Dziękuję bardzo. Bardzo proszę wszystkich państwa posłów obecnych na sali plenarnej, w innych salach, a także tych, którzy łączą się z nami zdalnie, o naciśnięcie dowolnego przycisku dla potwierdzenia uczestnictwa w posiedzeniu.

Stwierdzam kworum. Bardzo proszę. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Proszę o zarządzenie przerwy celem zwołania Konwentu Seniorów, abyście tam państwo zdecydowali o tym, że czas już skończyć z reglamentacją dostępu do tego miejsca, do sali posiedzeń plenarnych Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

To jest męczące, bezsensowne, jak cała ta koronopanika, pandemiopsychoza, której ofiary widzę także i w murach Sejmu Rzeczypospolitej. Czas z tym skończyć, czas wypuścić naród z kwarantanny. Chciałabym przypomnieć, że to nie jest moja decyzja.

Jest wniosek o przerwę, ale najpierw wysłuchamy innych. Bardzo proszę, panie pośle. Wysoka Izbo! Na podstawie art. 184 chciałbym złożyć wniosek o przerwę i zwołanie Konwentu Seniorów. Lewica chce, żebyśmy dzisiaj skorzystali z szansy, jaką daje spora pustka w dzisiejszym harmonogramie, i zajęli się czymś naprawdę istotnym. Proszę państwa, minął kolejny miesiąc. Tysiące ludzi dostały zwolnienia, tysiące ludzi trafia na bezrobocie. Mija kolejny miesiąc, a rząd nie zaproponował nic ludziom, którzy tracą pracę. Rząd nie zaproponował nic ludziom, którzy w tym momencie są skazani na głodowy zasiłek. Niedawno jeden z ministrów tego rządu popisał się brakiem wiedzy, nie umiał odpowiedzieć na pytanie, ile wynosi zasiłek. Minimalny zasiłek powinien wynosić 1400 zł na rękę, a zasiłek powinien, proszę państwa, stanowić połowę ostatniej płacy. To są normalne, europejskie standardy. W zeszłym tygodniu wspólnie z Robertem Biedroniem przedstawiliśmy stosowny projekt ustawy. Dziękuję bardzo. Kolejny wniosek o przerwę. Proszę. Chciałbym nietypowo, pani marszałek, podziękować za zrozumienie i w pewnym sensie wsparcie głosu, który dzisiaj na posiedzeniu Konwentu w imieniu klubu Koalicji zgłosił pan przewodniczący Budka. Mamy do czynienia z sytuacją bardzo niebezpieczną. Dzisiaj został opublikowany raport Narodowego Banku Polskiego, który mówi o prognozach i o polityce banków wobec rynku kredytowego. Mimo płynności banki przyjęły zasadę: ten, kto dostał pomoc w ramach tarczy, jakąkolwiek - żadnej pomocy, żadnych kredytów. Ktoś, kto prowadzi działalność gospodarczą, która w jakikolwiek sposób jest ograniczona z powodu koronawirusa przez rząd: fryzjerzy, zakłady fryzjerskie, kosmetyczki, ale i teatry, aktorzy, kina, sklepy, wszyscy, którzy mają jakiekolwiek restrykcje - żadnych kredytów. To zabije polską gospodarkę.

Zwróciłam się do pana premiera z taką prośbą i myślę, że na czwartek.

Ale już był wniosek formalny, panie pośle. Wysoka Izbo! Państwo jest w rozgardiaszu, państwo jest w rozsypce organizacyjnej. To jest całkowita kompromitacja obozu władzy, ale to jest również kompromitacja ram ustrojowych, które pozwalają na samowładztwo, które pozwalają na traktowanie obywatela jak poddanego, a nie jak gospodarza. Za 4 dni mają się odbyć wybory, a Polacy nie wiedzą, kto, gdzie, kiedy, jak, w jaki sposób. Trzeba doprowadzić do wprowadzenia stanu klęski żywiołowej, bo ta sytuacja to nie jest wina kandydatów. To nie jest nawet wina koronawirusa. To jest wina złych decyzji, zabrania kompetencji Państwowej Komisji Wyborczej, braku współpracy z samorządami i niewprowadzenia stanu klęski żywiołowej nie po to, żeby przenieść wybory, tylko żeby stwierdzić fakt. Dziś mieliśmy rozmawiać o funduszu płynności. Nawet tej ustawy nie potraficie od 3, 4 tygodni przygotować. Ogarnijcie się! O matko, panie pośle. Słyszymy wszyscy, naprawdę. Dziękuję bardzo. Tak naprawdę padł jeden wniosek, podwójny, o przerwę i ten wniosek poddam pod głosowanie. Bardzo proszę. Kto z pań i panów posłów jest za zarządzeniem przerwy w obradach, bardzo proszę o naciśnięcie przycisku.

Kto jest przeciw.

Stwierdzam, że Sejm wniosek odrzucił.

Ponieważ dzisiaj jest wielu posłów i obradujemy w 11 salach, po dyskusji stwierdziłam, że w każdej sali będziecie państwo mieli przedstawiciela Ośrodka Informatyki.

Taka też była, rozumiem, sugestia, żeby to wszystko przebiegało sprawnie, żeby każdy wiedział, jak ma się zalogować.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 13. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o kołach gospodyń wiejskich (druki nr 336 i 352) Proszę pana posła Roberta Telusa o przedstawienie sprawozdania komisji. Szanowna Pani Marszałek! Panie Premierze! Pani Minister! Mam zaszczyt przedstawić państwu sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o kołach gospodyń wiejskich, druk nr 336. Marszałek Sejmu, zgodnie z art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 regulaminu Sejmu, skierowała w dniu 15 kwietnia 2020 r. powyższy projekt ustawy do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi do pierwszego czytania. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi po przeprowadzeniu pierwszego czytania i rozpatrzeniu tego projektu ustawy na posiedzeniu w dniu dzisiejszym, tj. 5 maja 2020 r., wnosi, aby Wysoki Sejm uchwalić raczył załączony projekt ustawy. Takie krótkie sprawozdanie z tego, co działo się na posiedzeniu komisji rolnictwa.

To pokazuje, jak bardzo ważny jest to projekt, jak bardzo ważny jest to kierunek, który rząd Prawa i Sprawiedliwości, najpierw pani Beaty Szydło, później pana Mateusza Morawieckiego, rozpoczął.

Bardzo dziękujemy za to uzasadnienie, za przedstawienie tego projektu. Przede wszystkim projekt przewiduje powierzenie zadań ustawowych realizowanych dotychczas przez pełnomocnika rządu do spraw małych i średnich przedsiębiorstw pełnomocnikowi rządu do spraw lokalnych inicjatyw społecznych. Druga zmiana jest chyba bardziej oczekiwana.

Pochodzę z powiatu opoczyńskiego, drodzy państwo.

Druga zmiana, o której już mówiłem, to jest te 40 mln zł.

Pani marszałek, pozwoli pani, że powiem jeszcze dosłownie dwa zdania. Chodzi o głosy krytyczne, które mnie osobiście bardzo mocno zaskoczyły.

Dla rządu Prawa i Sprawiedliwości wszystkie sprawy są ważne.

Pani minister wytłumaczyła, że w tym momencie nie można takiej poprawki wprowadzić, bo to jest prognoza długoterminowa, którą można uwzględnić przy budżecie. Pani minister obiecała, że będzie robić wszystko, że będzie rozmawiała z panem przewodniczącym komisji finansów, jak również z premierem, żeby to wprowadzić w ramach prognozy długoterminowej. Dziękuję bardzo, panie pośle. Na przyszłość bardzo proszę trzymać się wyznaczonego czasu. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i koła. Jako pierwszy głos zabierze pan poseł Robert Telus w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Oczywiście myślę, że nikogo nie zaskoczę, jeżeli powiem, że klub Prawo i Sprawiedliwość w całości popiera ten projekt. Klub w całości popiera również kierunek, który objął rząd Prawa i Sprawiedliwości, czyli wspieranie kół gospodyń wiejskich na wsi.

I tutaj również chcę powiedzieć o jednej bardzo ważnej rzeczy.

Drodzy Państwo!

Nie jest to w żaden sposób polityczne.

Mówię to szczególnie do wójtów z PSL-u czy wójtów z Platformy Obywatelskiej, bo są tacy wójtowie, drodzy państwo, są tacy wójtowie. Mogę dać przykład, tylko nie chcę w tym momencie dawać przykładu na to, że atakują, że robią wszystko, żeby koła gospodyń wiejskich nie rejestrowały się w ARiMR i nie korzystały z tych środków.

Nie ma żadnej segregacji, jak niektórzy mówili na posiedzeniu komisji: że to jest segregacja, że tylko część kół może się zarejestrować, a część nie może skorzystać z tych środków.

Dziękuję bardzo, panie pośle. Stanowisko Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska przedstawi pani poseł Marzena Okła-Drewnowicz. Pani Marszałek! Pani Minister! Wysoka Izbo! Koła gospodyń wiejskich przetrwały wiele. Problem polega na tym, że państwo mówicie, że samorządowcy dyskryminują te koła gospodyń wiejskich, które idą do agencji, do waszego prezesa. Żaden samorząd nie dyskryminuje żadnego koła gospodyń wiejskich. Kobiety w kołach gospodyń są mądre i nie dadzą się uzależnić od kogokolwiek, a samorządowcy są z każdej opcji politycznej, od prawej strony do lewej, bo na tym polega samorządność. Natomiast Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - niech wybaczy pan poseł z Prawa i Sprawiedliwości - ma prezesa z państwa nominacji. Wielką niesprawiedliwością jest to, że wy w tej agencji dajecie pieniądze tylko i wyłącznie tym kołom, które do tej agencji pójdą i do tego prezesa pójdą. To jest bardzo niesprawiedliwe. Skoro szanujecie wszystkie koła gospodyń wiejskich, to dajcie pieniądze wszystkim kołom. Nie zmuszajcie ich do sztucznej rejestracji w agencji. Nie zmuszajcie ich do tego.

Do agencji z wnioskiem o rejestrację i dofinansowanie przystąpiło 500, jednak 300 nie przystąpiło.

Otóż jakoś tak dziwnie się składa, że zawsze o kołach gospodyń wiejskich przypominacie sobie tuż przed wyborami. Tak było tuż przed wyborami samorządowymi w 2018 r., tuż przed wyborami do europarlamentu w 2019 r. Jak to wyglądało w praktyce? Otóż w 2018 r. przeznaczyliście dla kół 90 mln. W ubiegłym roku przeznaczyliście 40 mln. Znowu koła gospodyń wykorzystały 29 mln. W tym roku mówicie o 40 mln. Nie dajcie tylko tym, którzy idą do agencji i do prezesa, tylko dajcie wszystkim.

To jest jedna rzecz. Zachęcałabym jednak państwa do tego, żebyście stworzyli taki mechanizm, który spowoduje, że te pieniądze będą co roku i będą jednakowe i uniwersalne dla wszystkich, na wzór choćby funduszu sołeckiego.

Oczywiście klub Koalicja Obywatelska będzie głosował za tym, żeby pieniądze trafiały do kół gospodyń wiejskich. Dziękuję bardzo, pani poseł. Stanowisko klubu parlamentarnego Lewica zaprezentuje pan poseł Robert Obaz. Bardzo proszę. Wysoka Izbo! W wypowiedzi posła sprawozdawcy zabrakło mi jednego zdania: słuszną linię ma nasza władza. Niczym Bareja w „Misiu” podkreślał on, jak to jest dobrze i jak to rząd Prawa i Sprawiedliwości traktuje wszystkich równo.

Jestem przekonany, że każdemu z nas powinno zależeć na budowie społeczeństwa obywatelskiego, które opiera się przede wszystkim na inicjatywie oddolnej, integrującej Polki i Polaków oraz angażującej ich na rzecz wzmacniania więzi społecznych, edukacji oraz poszukiwania optymalnych rozwiązań problemów lokalnych. Nie ulega wątpliwości, że jedną z niezwykle aktywnych grup w zakresie wspierania i rozwoju lokalnych społeczności stanowią niedocenione w sposób należyty przez rząd koła gospodyń wiejskich.

Dlatego tych 40 tys. organizacji ma prawo być równo traktowane. Chciałbym podkreślić, że wsparcie finansowe płynące do kół gospodyń wiejskich nie może opierać się na kalendarzu wyborczym, bo dzisiaj niestety tak to wygląda. Rok 2018 - wybory samorządowe, mamy wsparcie kół gospodyń wiejskich, 2019 r. - jesteśmy na piknikach, pan prezes wita się z wszystkimi paniami, panią Marysią, panią Zosią, a dzisiaj głosami posłów PiS-u poprawka dająca możliwość wspierania kół gospodyń wiejskich nie tylko w roku 2020, ale w kolejnych latach, zostaje przegłosowana negatywnie. Posługiwanie się środkami finansowymi na rzecz jedynie doraźnego wsparcia tych pożytecznych w skali lokalnej organizacji jest marnowaniem potencjału społecznego, jaki koła gospodyń wiejskich w ciągu ostatnich lat swojej działalności wypracowały. Jak pokazują badania, większość kół to organizacje w dużej mierze nastawione na działalność o niewielkim zasięgu i skupione przede wszystkim na najbliższym otoczeniu.

Jej członkowie często działają także w lokalnych organizacjach kół gospodyń wiejskich. W tym miejscu warto przypomnieć, bo wczoraj był dzień strażaka, że do dzisiaj rząd Prawa i Sprawiedliwości nie uchwalił obywatelskiego projektu ustawy dotyczącego dodatków do emerytur strażaków ochotniczej straży pożarnej, na którą czeka blisko 700 tys. członków tej organizacji. Biorąc to pod uwagę, należy zauważyć, że zaufanie społeczne, którym obdarzane są koła gospodyń wiejskich, charakteryzuje się wysokim stopniem budowania sieci społecznego zaangażowania, co nie tylko ułatwia im podejmowanie wspólnych działań razem z lokalną społecznością, ale przede wszystkim ułatwia im budowanie wokół swojej działalności kapitału społecznego, który integruje i wzmacnia więzi społeczne w lokalnej strukturze. O tym, jakie jest podejście i dlaczego te pieniądze miały być dane, dzisiaj na posiedzeniu komisji usłyszeliśmy chyba. Pani minister odpowiedziała: Ta zmiana podyktowana jest tym, by koła gospodyń wiejskich jak najszybciej otrzymały tę pomoc, szczególnie w tym trudnym czasie, w którym jesteśmy. Dostajemy wiele zapytań, np. czy będą mogły otrzymać środki na szycie maseczek w ramach walki z koronawirusem. Przepraszam bardzo, czy te pieniądze mają być przeznaczone - i taki jest argument, że musimy to szybko wprowadzić, bez przedłużenia na kolejne lata - tylko po to, żeby te panie szyły maseczki, bo polskiego rządu nie stać na to, żeby je kupić?

Wystąpienie w imieniu Klubu Parlamentarnego Koalicja Polska - Polskie Stronnictwo Ludowe - Kukiz15 przedstawi pani poseł Bożena Żelazowska. Bardzo proszę.

Szanowna Pani Marszałek! Pani Minister! Wysoka Izbo!

Jak ważną rolę odegrały koła gospodyń wiejskich w dziejach naszej ojczyzny, w której działają już od ponad 150 lat, nie muszę nikogo na tej sali przekonywać. Chcę z tego miejsca w imieniu koleżanek i kolegów z Koalicji Polskiej - Polskiego Stronnictwa Ludowego - Kukiz15 podziękować wszystkim paniom zaangażowanym w prace na rzecz społeczności lokalnej - działaczkom ludowym, nauczycielkom, gospodyniom domowym, lekarkom, twórczyniom, animatorkom kultury - za wielką pracę, jaką panie włożyły w rozwój swoich społeczności; pracowały panie na rzecz pomocy rodzinom wiejskim, pomagały w wychowaniu i kształceniu dzieci i młodzieży, działały na rzecz ochrony zdrowia. Organizacje kobiece mocno przyczyniły się do rozwoju edukacji i przedsiębiorczości kobiet. Mają ogromny wkład w rozwój i kultywowanie naszej historii i tradycji. Na co dzień spotykam się z paniami z kół gospodyń wiejskich w moim okręgu podwarszawskim, ale nie tylko, i wiem, jak mocno członkinie kół angażują się w integrację środowiska, w kultywowanie zwyczajów i tradycji narodowych. Widzę też, jak wraz ze zmianami społecznymi koła gospodyń wiejskich zmieniają formułę swojej działalności i świetnie sobie radzą w nowej rzeczywistości. Członkinie kół gospodyń wiejskich zawsze niezwykle ambitnie podejmują nowe wyzwania. Ich działalność była i jest powszechnie szanowana i ceniona. W imieniu klubu Koalicja Polska - Polskie Stronnictwo Ludowe - Kukiz15 chcę za tę pracę raz jeszcze serdecznie podziękować. Obecna nowelizacja jest już drugą nowelizacją ustawy o kołach gospodyń wiejskich. Ustawa powstała w listopadzie 2018 r. Pierwsza nowelizacja miała miejsce już w kwietniu 2019 r. Nie zmieniła tego, co jest najistotniejsze w tej ustawie. co dzieli środowiska wiejskie.

Proszę sobie wyobrazić, a państwo posłowie pewnie doskonale o tym wiecie, że koła, które miały ogromną historię i tradycję, które od wielu lat działały w danej miejscowości, miały tylko niecały miesiąc czasu, aby się zarejestrować. Wiemy, że w tym czasie przypadają święta Bożego Narodzenia, ale też była prowadzona cała akcja, aby właśnie się nie rejestrowały. I takich nowych kół jest dzisiaj 59%. Jeszcze jedną niekonstytucyjną kwestią, która jest zawarta w tej ustawie, jest kwestia członkostwa.

Raz jeszcze podkreślam: jest to kwestia bardzo ważna dla środowiska kół gospodyń wiejskich, dlatego że spotykając się z paniami, często słyszę, że zwracają one na to uwagę, że te koła, które nie zdążyły się wówczas zarejestrować, nie mogą korzystać z dofinansowania. Od tej pory mogą być zakładane koła w miastach do 5 tys. mieszkańców i w sołectwach, które leżą w granicach administracyjnych miast. Obecna nowelizacja utrzymuje kwotę 40 mln zł dla kół gospodyń wiejskich, a pamiętajmy, że w pierwszym roku na ten cel była przeznaczona kwota 90 mln. Otóż dotychczas była to funkcja pełnomocnika rządu do spraw małych i średnich przedsiębiorstw, który w pierwszej i drugiej wersji ustawy sprawował nadzór nad (Dzwonek) kołami, a w tej nowelizacji ma zostać zastąpiony przez pełnomocnika rządu do spraw lokalnych inicjatyw społecznych, który w myśl nowych zapisów mógłby we współpracy z prezesem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa powołać w celu aktywizacji wspólnot i społeczności lokalnych na obszarach wiejskich wojewódzkich koordynatorów. społeczności lokalnych powołany został rozporządzeniem z 14 stycznia tego roku. Tak że w imieniu Klubu Parlamentarnego Koalicja Polska - Polskie Stronnictwo Ludowe - Kukiz15 składam wniosek, aby wszystkie koła, które funkcjonują na terenach wiejskich i nie tylko, mogły otrzymywać dotacje. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję, pani poseł. Bardzo proszę.

Wysoka Izbo! Mówimy tutaj o kolejnej zmianie ustawy, o ustawie, która zmienia ustawę. Już ad rem. Same koła gospodyń wiejskich mają, umówmy się, bardzo długą tradycję, od 1866 r.

O tym należy cały czas pamiętać.

Tutaj jest wielka rola kulturotwórcza właśnie tych zrzeszeń, zwłaszcza dla kultury ludowej. Z reguły też promują one tradycje i promują normalną rodzinę. To jest taki przekaźnik, taki depozytariusz naszej kultury narodowej i zrozumiałe jest, że ze strony państwa będą wspierane te inicjatywy. Natomiast, na co warto zwrócić też uwagę, już w 2018 r. została wprowadzona ustawa dotycząca kół gospodyń wiejskich. Przewidziano konkretne dotacje na te koła gospodyń, bo mają też zadania jakby kobiece, ale można je porównać do ochotniczych straży pożarnych. W 2018 r. mieliśmy wybory. Wtedy została stworzona ta ustawa. W 2019 r. też mieliśmy wybory i wtedy powstała nowelizacja tej ustawy. W 2020 r. znowu mamy wybory i znowu powstaje nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich.

Trzeba to powiedzieć jasno.

Zachęcam do tego, aby to zmienić. Od początku tej kadencji żadna z poprawek Konfederacji nie przeszła przez Sejm. i wiemy, że jest to działanie polityczne, a więc zwracam się do rządu: zmieńcie to. Dziękuję bardzo, panie pośle. Bardzo proszę. Naprawdę trudno uwierzyć, że Rzeczpospolita potrzebuje prawa doprowadzonego do poziomu kółek rolniczych i kół gospodyń wiejskich. Za każdym razem, kiedy wydaje mi się, że już dogrzebujemy się do dna tego oceanu absurdu legislacyjnego, ktoś puka od spodu z takim właśnie pomysłem. Naprawdę im bardziej chory kraj, tym więcej w nim praw, taka jest prawda. Nie mam nic przeciwko - chyba nikt nie ma nic przeciwko - kołom gospodyń wiejskich, to są szacowne organizacje, z długą tradycją, chwała im, ale dlaczego, do cholery, nie mogą działać w oparciu o dokładnie takie same przepisy, w oparciu o jakie działają wszystkie inne stowarzyszenia w Polsce? Bo to do tego się sprowadza, że wszyscy płacimy składki na organizację, której często nie zobaczymy nigdy na oczy.

Nie dajcie się kupić za swoje pieniądze, bo każdy kij ma dwa końce. Kto daje, ten wymaga. Jeśli pozwolimy, żeby władza sprawiała wrażenie, że coś jej zawdzięczamy, że nas finansuje, to nie dziwmy się, że potem spróbuje nam na każdym kroku rozkazywać. Oczywiście jest to jedna wielka zbiorowa iluzja, ale tak to mniej więcej działa. Dzisiaj obiecuje gospodyniom, jutro będzie obiecywał górnikom, piłkarzom, artystom, akwarelistom i komuś jeszcze. A skąd weźmie dla akwarelistów, piłkarzy, górników i piekarzy?

Bo nie wiem, dlaczego zajmujemy się kołami gospodyń wiejskich, a nie kwadratami wiejskich gospodarzy albo miejskimi trójkątami. Czy wszystkie inne stowarzyszenia będziemy regulować tak samo? Dziękuję bardzo. Na tym kończymy oświadczenia. Przechodzimy do pytań.

Bardzo proszę. Wysoka Izbo! Oczywiście wszyscy macie rację, tylko to ewidentnie jest ustawa wyborcza: co rok w wybory się pojawia, co rok obiecuje się pieniądze. Nikt z nas nie ma wątpliwości, że koła gospodyń wiejskich chcą być samodzielne, dobrze finansowane i budżet państwa może im pomagać. Pani tak ładnie mówiła w komisji o tym, że państwo daliście impuls do działania kołom gospodyń wiejskich. Impuls miały one przez 120 lat, a państwo zniszczyli równowagę w tych kołach. Jeżeli w jednej wsi może być jedno koło i może ono dostawać pieniądze, a koło, które działa 120 lat i nie zarejestrowało się, nie dostanie pieniędzy, w jednej wsi - nie wiem, czy pani była - to naprawdę jest to nieuczciwe. Dzielicie Polaków nie tylko w miastach, ale i na wsiach, dzielicie Polaków tam, gdzie tylko się da, po to tylko żeby co roku tu przychodzić, panie pośle, i mówić: Teraz Prawo i Sprawiedliwość daje pieniądze i bądźcie wdzięczni, [[Dzwonek]] bo nikt inny nie dał.

Bardzo proszę. Wysoki Sejmie! Dowiedzieliśmy się na tej sali, że upodmiotowienie organizacji pozarządowej polega na jej afiliowaniu przy agencji rządowej. Pani pełnomocnik, miałaby pani zasługę, gdyby tą nowelą wprowadziła pani równość pomiędzy kołami gospodyń wiejskich, tzn. bez względu na to, w oparciu o jaki akt prawny się zarejestrowały, wszystkie mogłyby dostawać pieniądze.

Tak to wygląda. Dziękuję bardzo, panie pośle. Kolejne pytanie zada pani poseł Iwona Maria Kozłowska, Koalicja Obywatelska. Zapraszam, pani poseł. Wysoka Izbo! Tak jak już tu powiedziano, koła gospodyń działają od 150 lat, a pierwsze koło gospodyń o tej nazwie powstało w 1877 r. Na przełomie tych wszystkich lat koła gospodyń działały, wspierały, a jednocześnie jednoczyły społeczność wiejską. Koła gospodyń przekazują sobie, swoim pokoleniom i kobietom swoje doświadczenia i swoją wiedzę. Współpracują z radami sołeckimi, z ochotniczymi strażami pożarnymi i jednoczą całe społeczeństwo wiejskie.

Czy macie państwo już może listę tych koordynatorów? Czy są wyznaczone osoby, które będą tymi koordynatorami, i jakie zadania, pani minister, mają wykonywać ci koordynatorzy? Jaka też będzie kwota, którą państwo wykorzystacie na opłacenie tych koordynatorów (Dzwonek), i jakie to będą pieniążki, które zostaną przeznaczone na sfinansowanie tych zadań? Kolejne pytanie zada pani poseł Joanna Frydrych, Koalicja Obywatelska. Bardzo proszę. Wysoka Izbo! Pomoc finansowa dla kół gospodyń wiejskich jest bardzo istotna. Koła gospodyń wiejskich to organizacje kultywujące tradycję i lokalne zwyczaje, bardzo potrzebne i głęboko zakorzenione w lokalnej społeczności. Nikt nie sprzeciwia się przekazaniu środków pieniężnych dla tych organizacji. Ale czy konieczne jest tworzenie kolejnego organu administracyjnego, jakim jest pełnomocnik rządu do spraw lokalnych inicjatyw społecznych, czyli kolejny sekretarz bądź podsekretarz w ministerstwie polityki regionalnej? W środku epidemii mówicie państwo o cięciach w administracji, bo doskonale zdajecie sobie sprawę z deficytu budżetowego oraz tego, że są grupy społeczne, którym obecnie należy pomóc. Ale z drugiej strony tworzycie nowe organy w celu obsadzania swoimi ludźmi. I moje pytanie brzmi przede wszystkim tak: Czy dotychczasowy pełnomocnik nie dbał właściwie o koła gospodyń wiejskich i o inne inicjatywy społeczne? Dziękuję, pani poseł. Pani poseł Mirosława Nykiel, Koalicja Obywatelska. Bardzo proszę. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Projekt ustawy zakłada wspieranie kół gospodyń wiejskich - tylko kół gospodyń wiejskich. A przecież wiemy, że w gminach wiejskich i miejskich działa wiele organizacji pozarządowych, które wykonują zadania zarówno za samorząd, jak i za państwo i też czekają na takie wsparcie. Czy planujecie uruchomić takie wsparcie również dla tych innych działających organizacji pozarządowych? Ustawa powołuje też regionalników... regionalnych pełnomocników.

Pani poseł Marta Wcisło, Koalicja Obywatelska.

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Szanowni Państwo! Koła gospodyń wiejskich od 150 lat wpisują się w mapę kulturalną inicjatyw oddolnych polskiej wsi. Ale nie mogę zrozumieć, jak bardzo niesprawiedliwe, niewłaściwe i tendencyjne jest dzielenie jednej wsi na lepszych i gorszych, na koło gospodyń wiejskich, które zostało zarejestrowane na podstawie ustawy z 2018 r., i koło gospodyń wiejskich, które działa przykładowo 60 lat. Te kobiety od lat pielęgnowały, wspierały, rozwijały i pomagały kulturze, tradycji. Dziś nie dostają wsparcia i finansowania. Dlaczego koło gospodyń wiejskich w gminie Zakrzówek w miejscowości Majdan-Grabina, które dzisiaj obchodzi 60 lat, nie dostanie tego wsparcia, a koło w tej samej wsi, które jest zarejestrowane od roku, dostanie? Dzielicie sąsiadów, dzielicie Polaków. Bardzo proszę. Wysoka Izbo! W Polsce działa ok. 21 tys. kół gospodyń wiejskich skupiających ponad 1 mln kobiet. Swoimi działaniami odebraliście im niezależność i uzależniliście możliwość uzyskania wsparcia finansowego od rejestracji w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, pozostawiając te niezarejestrowane bez żadnej pomocy. Teraz chwalicie się kolejnymi przeznaczonymi pieniędzmi, lecz nadal nie potraficie rozwiązać ich realnych problemów. Dlaczego dzielicie koła gospodyń wiejskich? Panie mają do was duży żal za uszczęśliwianie ich na siłę, ale wybiórczo. Kobiety słusznie skarżą się, że w jednej wsi może działać tylko jedno koło. Uniemożliwiliście zaangażowanie się w członkostwo w kole działającym w innej miejscowości. Nie mówiąc już o biurokracji, z którą przyszło im się zmierzyć. Mam pytanie: Jaki jest cel powierzenia zadań realizowanych dotychczas przez pełnomocnika rządu do spraw małych i średnich przedsiębiorstw pełnomocnikowi rządu do spraw lokalnych inicjatyw społecznych? Po co utworzyliście w styczniu br. to stanowisko? Czyżby kolejne miejsce dla Pisiewiczów? Pani poseł Klaudia Jachira, Koalicja Obywatelska. Panie Szeregowy Pośle Kaczyński! Wysoka Izbo! Doceniam każdą inicjatywę, która sprzyja integracji kobiet i sprawia, że kobiety mogą wymieniać się swoim doświadczeniem i wspierać się. Ale mam nadzieję, że te dodatkowe fundusze sprawią, że kobiety będą mogły jeszcze bardziej wykorzystać ten potencjał. Może to czas, by właśnie tego typu organizacje promowały wśród kobiet regularne badania cytologiczne i mammograficzne. Może powinny być też miejscem, gdzie kobieta znajdzie wsparcie, gdy jest ofiarą przemocy w rodzinie albo gdy zmaga się w domu z chorobą alkoholową. W miastach jest dużo łatwiej o taką pomoc, dobrze o tym wiemy, mamy liczne prokobiece NGOs, które swoją drogą państwo odcinają od finansowania. Ale na wsi jest trudniej. Koła gospodyń wiejskich mogą zmienić pokutującą u nas niechlubną zasadę: nie mów nikomu, co się dzieje w domu. Kilka dni temu prawie jednogłośnie (Dzwonek) przyjęliśmy dobrą ustawę przeciwdziałającą przemocy, więc idźmy krok dalej. Dziękuję. Bardzo proszę. Pani Marszałek! Pani Minister! Wysoka Izbo! Cieszy mnie fakt, że rząd proponuje przeznaczyć choć 40 mln zł pomocy finansowej dla kół gospodyń wiejskich w tym roku. To ważne, aby te centra rozwoju lokalnych społeczności były dofinansowane. Ale jednocześnie smuci fakt, że to dofinansowanie przychodzi tak późno, prawie w połowie roku, i zaledwie 5 dni przed wyborami, co rodzi podejrzenie, że środowisko kół gospodyń wiejskich jest być może kolejnym środowiskiem, które rząd PiS traktuje instrumentalnie. Dlatego pytam: Czy próbujecie państwo tym gestem kupić głosy kobiet z kół gospodyń wiejskich, aby głosowały na waszego kandydata na prezydenta? A jeżeli nie, to czy pani minister może nam obiecać, że zwiększy limit wydatków z budżetu państwa na rozwój kół gospodyń wiejskich w ramach corocznego budżetu, tak jak w normalnych krajach? Pani minister, proszę odpowiedzieć szczerze: Czy to jednorazowa przedwyborcza kiełbasa, czy realne, stałe wsparcie? Bardzo proszę. Bardzo dziękuję. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Rząd ustami pani minister był uprzejmy zauważyć, że dał impuls do działania kół gospodyń wiejskich. Ja bardzo bym prosił panią minister o przedstawienie na piśmie wykazu tych kół, które trzeba było aktywizować. Jak mówię, na piśmie, żeby później nic nie uciekło. Jestem z południa i w moim powiecie, powiecie bielskim, w Bielsku-Białej, w powiatach cieszyńskim, żywieckim i pszczyńskim działa kilkadziesiąt kół i one naprawdę tak działają, że można by pewnie obdzielić działalnością tych kół szereg innych kół z terenu całej Polski.

Drugie pytanie.

Pytanie do pani minister, do rządu: Kiedy rząd skończy z dyskryminacją tych pań, które działają nie w politycznych kołach powołanych zarządzeniem, ustawą Prawa i Sprawiedliwości, ale w kołach, które działają w Polsce od 150 lat? Dziękuję bardzo. Ustawą sejmową, panie pośle. Bardzo proszę.

Szanowna Pani Marszałek! Pani Minister! Każda pomoc, która trafia do obywateli, którzy potrafią się zorganizować i wykonać ogrom lokalnych zadań na rzecz najbliższej społeczności, jest warta uwagi, warta wsparcia. Ale polscy obywatele, szczególnie ci, który się organizują, nie mogą być traktowani różnorodnie. Dlatego zadaję pytanie: Dlaczego koła gospodyń wiejskich, które są zarejestrowane jako stowarzyszenia, są pozbawione możliwości uczestnictwa w konkursach ogłaszanych przez ARiMR? To jest nierówne traktowanie Polaków, czyli podmiotów, które funkcjonują. Również one są pozbawione możliwości uczestniczenia w tych konkursach. Ich zadania są bardzo zbliżone. A co z aktywnością osób, które, szczególnie w większych wsiach, decydują się na założenie kilku kół gospodyń wiejskich? Przecież wsie są różnorodne. Ostatnie pytanie. Jest taka inicjatywa na Dolnym Śląsku, w gminie Osiecznica, we wsi Tomisław i Osieczów - powstało tu pierwsze stowarzyszenie: koło chłopa jako odpowiedź na aktywizację.

Bardzo proszę. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Często pojawia się pytanie: W ilu autobusach można zmieścić rząd Mateusza Morawieckiego? Prawidłowa odpowiedź: w trzech, ponieważ właśnie, Wysoka Izbo, powróciliście państwo do rekordu Beaty Szydło - 121 członków rządu Mateusza Morawieckiego. Dzisiaj dowiedzieliśmy się tak naprawdę, myślę, że większość z państwa, że mamy pełnomocnika rządu do spraw lokalnych inicjatyw społecznych. To jest, rozumiem, pani wiceminister, tak? Nie wiem, czym ta funkcja różni się od funkcji pełnomocnika rządu do spraw społeczeństwa obywatelskiego, bo to właśnie temu pełnomocnikowi podlegają lokalne inicjatywy społeczne. Szanowni Państwo! Chciałbym zwrócić uwagę również na to, że ta ustawa sortuje. Ta ustawa sortuje koła gospodyń wiejskich, które od 150 lat [[Dzwonek]] walczą o prawa kobiet. Walczą również o to, żeby w sposób godny. Wywalczyły sobie miejsce w społeczeństwie, wspierając je, edukując je, a dzisiaj tak naprawdę część z nich zostaje pozbawiona środków finansowych: wyłącznie te osoby i wyłącznie te podmioty, które zarejestrowały się w agencji, będą takie wsparcie otrzymywać. Pan poseł Grzegorz Braun, Konfederacja. Bardzo proszę.

Rzeczywiście zasadne jest pytanie o gospodarzy, zasadne jest pytanie o ludzi innych zajęć, mających inne miejsce zamieszkania, ale wy, żoliborscy socjaliści, kontynuujecie tę tradycję. Tu zwracam się do wszystkich dobrych patriotów, którzy tak się nasładzają tymi kołami gospodyń wiejskich. Ta tradycja wywodzi się od nieszczęśnicy imieniem i nazwiskiem Filipina Płaskowicka, towarzyszki Waryńskiego.

To jest wasza tradycja. Kiedy przymierzycie się do tego, żeby zaktywizować gospodynie miejskie? Co z tymi gospodarzami, którzy już się aktywizują i czują się dyskryminowani? Dziękuję bardzo, panie pośle. Bardzo proszę. Szanowna Pani Marszałkini!

Czas płynie, pani poseł. Kobiety wiejskie to sól ziemi. Od 150 lat zrzeszają się w kołach gospodyń wiejskich, które dbają o życie społeczne i kulturalne. Są ostoją lokalnej wspólnoty. Koła gospodyń wiejskich potrzebują wsparcia ze strony państwa. Ale tu pojawiają się pytania. Dlaczego zamiast wprowadzić systemowe wsparcie kół gospodyń wiejskich, rząd udziela im tylko jednorazowych form doraźnej pomocy? Dlaczego tę doraźną pomoc otrzymują tylko koła zarejestrowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a nie te funkcjonujące od dawna w ramach kółek rolniczych? To jawna dyskryminacja licznych kół gospodyń wiejskich działających w takiej formule często od wielu lat. Dlatego pytam, pani minister, czy rozszerzycie pomoc na wszystkie koła gospodyń wiejskich, bez względu na to, kiedy powstały i w jakiej formule funkcjonują, bez dyskryminacji?

Wszystkie kobiety zasługują na pomoc i wsparcie ze strony państwa - równo, sprawiedliwie i bez dyskryminacji. Dziękuję bardzo, pani poseł. Bardzo proszę. Pani Marszałek! Wysoki Sejmie!

One odgrywają bardzo ważną rolę. Państwo przez stworzenie odpowiednich mechanizmów wsparcia nie powinno ich dzielić. Liczy się aktywność na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego. To dobrze, że państwo wspomaga. Źle, że państwo dzieli ze względu na formułę prawną dostęp do środków publicznych. Tam wręcz odwrotnie, namawia się grupy niesformalizowane: chodźcie, twórzmy społeczeństwo obywatelskie, realizujmy określone projekty na rzecz jego aktywizacji, korzystając z osobowości prawnej innych podmiotów. Tu nie, zamknięto. Pytanie do pani minister: Jaką rolę będą odgrywali koordynatorzy? Ustawa przewiduje możliwość ich powołania. Dziękuję. Dziękuję, panie pośle. Bardzo proszę. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Koła gospodyń wiejskich od blisko 150 lat troszczą się o polską tradycję i aktywizują lokalne społeczności. Orzechowo, Brodowo, Sampława - to przykłady wsi, gdzie kobiety wzięły los lokalnej społeczności w swoje ręce. Jednocześnie koła gospodyń wiejskich przekazują lokalną tradycję turystom odwiedzającym obszary wiejskie. Chylę czoła przed naszymi gospodyniami. Państwo powinno wspierać ich działalność, ale także konsultować zasady wsparcia z zainteresowanymi podmiotami. Nawet w trudnym czasie władza nie może rezygnować z dialogu ze społeczeństwem obywatelskim. Stąd moje pytanie: Dlaczego nie przeprowadzono konsultacji społecznych z kołami gospodyń wiejskich i z innymi zainteresowanymi podmiotami? Niestety nie wszystkie lokalne aktywistki na obszarach wiejskich mogły skorzystać z pomocy państwa. Dotyczy to szczególnie kół działających w ramach kółek rolniczych. Stąd moje drugie pytanie: Dlaczego ustawa obejmuje pomocą tylko wybrane koła gospodyń wiejskich, pomija inne, często nie mniej zasłużone? Proszę o odpowiedź na piśmie, pani minister. Dziękuję bardzo, panie pośle. Pani poseł Paulina Matysiak, klub Lewica. Bardzo proszę. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Na wstępie powiem krótko: dobrze, że w tej sali wspomniano Filipinę Płaskowicką. Powinniśmy tutaj częściej przywoływać działaczki społeczne i socjalistyczne. Powiem natomiast odnośnie do samej ustawy, że jest to kolejna w ostatnim czasie nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich. Wydaję się, że jej zamiary i przepisy są słuszne, ale jednak jest kilka „ale”, ponieważ ona nie znosi największego problemu kół, czyli zbyt dużych wymogów biurokratycznych. Koła gospodyń wiejskich działają często nieformalnie, a jeżeli są już zarejestrowane, podlegają licznym wymogom formalnym. Muszą posługiwać się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, są zarejestrowane w KRS, a także w agencji restrukturyzacji. Była o tym już dzisiaj mowa. Moje pytanie brzmi: Czy nie czas wreszcie rozwiązać podstawowy problem kół, czyli stworzyć jednolitą, prostą i przejrzystą strukturę i procedurę rejestracji (Dzwonek) i obsługi formalnej tych kół, aby prawo nie było przeszkodą i utrudnieniem, tylko wspierało i zachęcało do ich zakładania i funkcjonowania? Dziękuję. Dziękuję, pani poseł. Pan poseł Marek Polak, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W przeciwieństwie do niektórych moich przedmówców pragnę na wstępie wyrazić swoją pełną aprobatę tego projektu, który jest kolejną dobrą propozycją rządu, mającą na celu ułatwienie funkcjonowania i realizacji zadań przez koła gospodyń wiejskich. To organizacje, które, jak wiemy, mają istotny wpływ na poprawę sytuacji społeczno-zawodowej kobiet, a także ich rodzin, i to nie tylko na obszarach wiejskich, ale także na terenach małych miasteczek. Koła gospodyń wiejskich, jak wszyscy wiemy, realizują swoje cele i zadania, w nieoceniony sposób pielęgnują i zachowują nasze zarówno narodowe, jak i regionalne tradycje, co jest niezwykle ważne.

Dlatego chciałem zapytać, czy zdaniem pana ministra przewidziane na rok bieżący środki w wysokości 40 mln zł będą wystarczające. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie pośle. Z kolejnym pytaniem zapraszam pana Dariusza Klimczaka, Polskie Stronnictwo Ludowe - Kukiz15. Bardzo proszę. Wysoka Izbo! Teraz próbuje podzielić na te koła, które są nowe, na te, które są stare, na te, które są zarejestrowane, na te, które nie są zarejestrowane, na te koła, które mają pieniądze, i na te koła, które nie mają pieniędzy. Czy budżet ministerstwa rolnictwa jest aż tak mały, czy bardziej chodzi o to dzielenie? Dlaczego chcecie ingerować w historię kół gospodyń wiejskich?

Między bajki można włożyć próby uniezależniania KGW od wójtów, bo wszyscy wiedzą, że od lat wójt, samorząd gminny były wsparciem dla KGW, OSP i odwrotnie. Gmina nigdy nie mogłaby wręcz funkcjonować bez dobrego ich funkcjonowania. Tak było w powiecie łowickim, tak było w tomaszowskim, tak było w wielu innych powiatach. Bardzo proszę, panie pośle. Szanowna Pani Marszałek! Pani Minister! Wysoka Izbo! Ustawa z listopada 2018 r. dała wiele nowych możliwości w zakresie rejestrowania i funkcjonowania kół gospodyń wiejskich. Te liczby, o których mówił pan poseł sprawozdawca, naprawdę robią imponujące wrażenie. Wtedy prawie 6 tys. kół gospodyń wiejskich zostało zarejestrowanych w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. To powiat niewielki, 40-tysięczny, sześć gmin wchodzi w skład tego powiatu.

Dziękuję, panie pośle. Bardzo proszę. Przy okazji dyskusji o roli i znaczeniu działalności kół gospodyń wiejskich chciałbym podkreślić bardzo ważny obszar życia społecznego na wsi - to jest problem samoorganizacji, aktywnego udziału w kształtowaniu tej rzeczywistości przez mieszkańców wsi. Myślę tu nie tylko o kołach gospodyń wiejskich, ale także o ochotniczych strażach pożarnych, o ludowych zespołach sportowych czy o kółkach rolniczych. Oczywiście mówimy o kołach gospodyń wiejskich, których rola i wkład w podtrzymywanie tradycji, w organizację życia kulturowego, wychowanie dzieci i kształtowanie takiej atmosfery są wyjątkowe. Myślę, że za to należą im się ogromne podziękowania. Tak się składa, że mam przyjemność obserwować tę aktywność, i wiem, jak ona jest ważna dla mieszkańców wsi. Myślę jednak, że [[Dzwonek]] samorządy są bardzo otwarte i wszystkie samorządy działają na rzecz wspierania w swojej aktywności struktur na terenie gminy, natomiast agencja chyba trochę urządowiła koła gospodyń wiejskich, choć nie powinna tego robić, bo jest to instytucja, która ma akredytację unijną i musi przestrzegać pewnych procedur i zasad, jeśli chodzi o wspieranie wszystkich aktywności. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Zanim oddam pani poseł głos, mam wielką prośbę do pań i panów posłów - o ograniczenie rozmów na sali plenarnej, ponieważ gdy jest nas tak mało, to dźwięk bardzo się niesie i bardzo przeszkadza osobom, które zadają kolejne pytania. Szanujmy się nawzajem. Bardzo proszę, pani poseł. Pani Marszałek! Na tej sali padło bardzo wiele ciepłych słów o zasługach kół gospodyń wiejskich, o ich tradycji, o ich działalności na rzecz społeczności lokalnych, ale okazuje się, że to jest za mało. Aktywność społeczna działaczek na terenach wiejskich jest mniej lub więcej warta. Jedne takie wsparcie dostaną - taka jest propozycja w ustawie - a inne nie. Dlatego nasuwają mi się pewne wątpliwości i konkretne pytania. Ile kół gospodyń wiejskich funkcjonowało na terenie Polski przed wprowadzeniem ustawy, jeżeli chodzi o koła rejestrowe i nierejestrowe, a ile kół zarejestrowanych w ARiMR to koła nowe?

Dziękuję. Dziękuję, pani poseł. Bardzo proszę. Pani Marszałek! Pani Minister! Wysoka Izbo! Reprezentując województwo podlaskie, chciałbym zadać dwa następujące pytania: Jaki zakres obowiązków mają koordynatorzy wojewódzcy, o których jest mowa w ustawie? Czy stanowisko koordynatorów wojewódzkich finansowane będzie z puli pieniędzy, którą przewiduje ustawa? Na koniec chciałbym zwrócić się z ogromną prośbą, żebyśmy nie dzielili kół na zarejestrowane i niezarejestrowane, tylko potraktowali je jednakowo. Dziękuję, panie pośle. Bardzo proszę. Pani Marszałkini! Wysoka Izbo! Moje pytania: Czy koła gospodyń wiejskich zgłaszały własne uwagi i zastrzeżenia do ustawy? Jeśli tak, to jakie to były zastrzeżenia? Proszę o odpowiedź na piśmie. Dlaczego nie zostały przeprowadzone konsultacje w sprawie procedowanej ustawy? Stan epidemiczny nie zwalnia z ich przeprowadzenia. I dołączam się do tego pytania, które padało już wielokrotnie. Polska prawica tak często powołuje się na znaczenie tradycji. Dlaczego więc koła gospodyń wiejskich o najdłuższej tradycji są dyskryminowane? Czy może dlatego, że założyła je socjalistka? Dziękuję, pani poseł. I pani poseł Bożena Żelazowska, klub Polskie Stronnictwo Ludowe - Kukiz15. Bardzo proszę. Pani Minister! Wysoka Izbo! Czy nowelizacja ustawy zlikwiduje wreszcie podziały, jakie powstały w środowiskach wiejskich? Czy w dzisiejszej dobie są potrzebni kolejni pełnomocnicy rządu ze swoim uposażeniem, biurem, całym zapleczem, kolejni koordynatorzy wojewódzcy i kolejne środki na ten cel? Natomiast moje pytania brzmią: Dlaczego środki przeznaczone na działalność kół w trzecim roku funkcjonowania ustawy nie zostały zaplanowane w budżecie, tylko wciąż pochodzą z rezerwy?

W ramach jakich struktur mieliby oni działać, skoro dzisiaj w każdym oddziale regionalnym są wyznaczeni opiekunowie KGW i to raczej wystarcza, bo jest ich 362? Czy rząd przeprowadził analizę, czy może audyt, na co zostały spożytkowane środki z lat poprzednich? W ustawie zapisano. że na cele statutowe. Dziękuję bardzo. Lista posłów zapisanych do głosu została wyczerpana. W imieniu rządu na pytania odpowie sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej pani minister Anna Gembicka. Bardzo proszę.

Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Projekt ustawy o zmianie ustawy o kołach gospodyń wiejskich to projekt oczekiwany przez osoby działające na rzecz wsi, kultury i tradycji. Koła gospodyń wiejskich na mocy ustawy sprzed 2 lat zyskały osobowość prawną i szereg ułatwień w swojej działalności. Państwo wszystko sprowadzacie do pieniędzy, tymczasem koła zyskały osobowość prawną, zyskały liczne ułatwienia: zwolnienia podatkowe, ułatwienia w rozliczaniu, w sprzedaży produktów.

Dzisiejszy projekt dotyczy z jednej strony powierzenia zadań wynikających z ustawy pełnomocnikowi rządu do spraw lokalnych inicjatyw społecznych, z drugiej strony natomiast - udzielenia pomocy w wysokości 40 mln zł. Padło wiele pytań, na jakiej podstawie te środki zostały oszacowane. Dysponujemy danymi od 2018 r., na podstawie których możemy określić, jaki jest przyrost wśród kół gospodyń wiejskich. Oczywiście prowadzimy też działania promujące i działanie edukacyjne, bo niestety ze strony wielu osób, które zwalczają koła gospodyń wiejskich.

Dysponują moim numerem, w razie wątpliwości się ze mną kontaktują. Naprawdę to jest bardzo przykre, kiedy dzwoni do mnie pani, która mówi, że usłyszała od wójta, że jak się zarejestruje, to żadnych pieniędzy nie dostanie, bo wcześniej było tak, że wójt z jednej z partii, która tutaj najgłośniej krzyczała, dawał pieniądze dla kół, owszem, tylko trzeba je było wydać w sklepie jednego z działaczy tej partii.

Jest wiele takich sytuacji, w których np. panie proszą o spotkanie praktycznie pod osłoną nocy, bo się boją, że wójt będzie się mścił. Powiem szczerze: dla mnie to jest nie do zaakceptowania. Albo takie głosy, które panie słyszą od działaczy kółek rolniczych, że nie będą zapraszane na dożynki za to, że się zarejestrowały. Powiem szczerze: dla mnie to jest nie do pomyślenia. Nie wiem, czy państwo spędzacie dużo czasu na wsi, ale ja akurat jestem z takiej małej wioski i wiem, że akurat dożynki to jest jedno z najważniejszych świąt dla rolników, a także dla tych właśnie osób, które działają w kołach gospodyń wiejskich. I to jest bardzo przykre, że właśnie próbuje się kołom zabraniać, żeby pojawiały się na takich wydarzeniach. Odnosząc się do tych różnych pytań - większość niestety nie dotyczyła w ogóle tego projektu ustawy - po pierwsze, chcę powiedzieć, że nikt nie twierdzi, że koła gospodyń wiejskich powstały w 2018 r. Wszyscy dobrze wiemy, że one funkcjonują, niektóre mają ponad 100-letnią tradycję, ale niektóre powstały w ostatnich latach. Myślę, że powinniśmy doceniać obydwie te formy, zarówno te koła z ogromną tradycją, jak i te koła nowe, które zaktywizowały się teraz.

To są kompletne bzdury. Ustawa też nie przewiduje utworzenia urzędu pełnomocnika do spraw lokalnych inicjatyw społecznych. To wynika z samego tekstu ustawy.

To jest kilkaset milionów złotych. Upewniliśmy się, że koła gospodyń wiejskich także mogą z tego wsparcia korzystać, bo to nie jest tylko możliwość uzyskania tych 3 tys. zł, ale to jest także możliwość korzystania z różnego rodzaju dotacji, konkursów, które są prowadzone np. przez Narodowy Instytut Wolności. Pełnomocnicy w agencjach restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa funkcjonują (Dzwonek) już od 2 lat. To nie jest nowy urząd, więc tutaj też chciałabym od razu sprostować, że nie tworzymy żadnych nowych urzędów. Kolejne pytanie. Jeśli chodzi o te zadania, które koła gospodyń wiejskich realizują, przygotowujemy ustawę i rozporządzenie w taki sposób, żeby ta swoboda wydawania środków była jak najszersza. Nie chcemy narzucać, że macie wydać na ten konkretny cel, bo panie działające na wsi dobrze wiedzą, na co mają wydać te pieniądze, i nie jest im też potrzebny ktoś, kto będzie nad nimi w jakiejś organizacji i będzie im mówił, że mają tutaj zapłacić składkę, a tutaj mają wydać to na taki i taki cel. One bardzo dobrze wiedzą, na co te pieniądze wydać, i takie pouczenia są absolutnie niepotrzebne. Pan poseł Braun powiedział, że mężczyźni są dyskryminowani. Mężczyźni też mogą się zapisywać do kół gospodyń wiejskich, więc chciałam. Kolejna sprawa.

Te rozwiązania są przystosowane do charakteru ich działalności. Mamy w trzecim sektorze różnego rodzaju organizacje: mamy stowarzyszenia zwykłe, mamy stowarzyszenia zarejestrowane w KRS-ie, mamy fundacje, mamy koła gospodyń wiejskich, część osób działa nieformalnie. Te wszystkie formy prawne między sobą się różnią, ale co najważniejsze, one są dostosowane do ich charakteru działania i każda z tych form łączy w sobie pewne prawa i pewne obowiązki.

Kończąc już, chciałabym z tego miejsca podziękować wszystkim paniom i panom, którzy działają w kołach gospodyń wiejskich. Robicie naprawdę wspaniałe rzeczy.

Dziękuję bardzo, pani minister. Ale bardzo proszę, panie pośle, trzymać się czasu, bo mamy już duże opóźnienie. Szanowna Pani Marszałek! Szanowna Pani Minister! Przede wszystkim były takie pytania, dlaczego każemy rejestrować się w ARiMR. To jest taka normalna rzecz.

Tu jest ta sama sytuacja, że trzeba się zarejestrować w ARiMR. Drodzy państwo, nikogo nie dzielimy. Wszystkie koła gospodyń wiejskich: i te, w których działają mężczyźni, i te, w których działają kobiety, wszystkie koła gospodyń wiejskich mogą.

To państwo próbujecie dzielić. Wszystkie mogą. Drodzy państwo z Platformy Obywatelskiej, którzy powołujecie się na fundusz sołecki, chcę przypomnieć wszystkim, nie wszyscy byli wtedy w Sejmie w 2009 r., że to nasza ustawa, Prawa i Sprawiedliwości, której miałem przyjemność być wnioskodawcą, była złożona jako pierwsza, a wasza była po pół roku i wspólnie nasze ustawy były uchwalone, tak że to był nasz pomysł: fundusz sołecki, i dobrze, że taki jest, bo on jest bardzo potrzebny i bardzo dobrze działa. To ja proponuję pani poseł, która tu mówiła o tej biurokracji, żeby spróbowała zarejestrować to koło gospodyń wiejskich jako stowarzyszenie i wtedy zobaczy, jaka to jest biurokracja, i wtedy zobaczy, jakie to jest udogodnienie, że wprowadzamy tę ustawę, że wprowadziliśmy tę ustawę, żeby właśnie nie było tej biurokracji. I drodzy państwo, cały czas jedna rzecz: że ustawa przed wyborami. No, drodzy państwo z Platformy Obywatelskiej i z Polskiego Stronnictwa Ludowego, przypominam, że rządziliście przez 8 lat i przez 8 lat nie daliście dla kół gospodyń wiejskich złotówki. Jednej złotówki nie daliście przez 8 lat. A teraz nam wymawiacie, że my dajemy co roku, i to tyle, ile jest potrzeba, 16, 29 i w tej chwili 40 mln zł? I wy mówicie, że przed wyborami? Drodzy państwo, was nie było stać ani na 500+, ani na 300+, ani na dofinansowanie komunikacji, ani na tworzenie Poczty Polskiej na wsiach, ani na tworzenie. żadne programy dla ludzi mieszkających na wsi, na komunikację.

zwykłym rodzinom. Drodzy państwo, sprawa wójtów. Tutaj już pani minister o tym powiedziała. Ale są wójtowie, którzy naprawdę robią wszystko, żeby się koła gospodyń wiejskich nie rejestrowały.

Polacy wiedzą, na co wydawać środki, i Polacy wydają te środki tak, żeby skorzystały na tym właśnie zwykłe rodziny, żeby na tym skorzystały obszary wiejskie, i tak, żeby to społeczeństwo obywatelskie, na które wy się tak pięknie powołujecie, funkcjonowało. My wierzymy kołom gospodyń wiejskich [[Dzwonek]] i my będziemy wspierać koła gospodyń wiejskich, bo one są dla nas, dla Polski bardzo ważne. W związku z tym, że w czasie drugiego czytania zgłoszono do przedłożonego projektu ustawy poprawki, proponuję, aby Sejm skierował ponownie ten projekt do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w celu przedstawienia sprawozdania. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 11. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (druki nr 207 i 351) Proszę panią poseł Ewę Szymańską o przedstawienie sprawozdania komisji. Bardzo proszę. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw, druk nr 207. Sejm na 5. posiedzeniu w dniu 12 lutego 2020 r. zgodnie z art. 39 ust. 2 regulaminu Sejmu skierował powyższy projekt ustawy do Komisji Finansów Publicznych w celu rozpatrzenia. Komisja Finansów Publicznych rozpatrzyła powyższy projekt ustawy na posiedzeniach w dniach 13 lutego i 5 maja, a podkomisja stała do spraw monitorowania systemu podatkowego - w dniu 11 marca 2020 r. W komisji rozpatrzono złożone poprawki, szeroko dyskutowano o tym projekcie.

Dziękuję. Stanowisko Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość przedstawi pan poseł Piotr Polak. Bardzo proszę. Dziękuję. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość mam zaszczyt przedstawić nasze stanowisko w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw, druki nr 207 i 351. Wysoka Izbo! Przedłożony projekt ustawy wprowadza zmiany w kilku ustawach, a mianowicie w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, tzw. ustawie o PIT, ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawie o CIT, Ordynacji podatkowej, ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ustawie o podatku od towarów i usług, tzw. ustawie VAT-owskiej, ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawie o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. Zmiany, które są zawarte w tym projekcie, w drukach nr 207 i 351, są to zmiany, które dostosowują przepisy o podatku dochodowym do nowej Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Te zmiany również ograniczają liczbę rocznych obliczeń podatku PIT-40A sporządzanych przez organy rentowe dla podatników, u których z obliczenia organu rentowego wynika nadpłata podatku, oraz są to przepisy kompleksowo regulujące kwestie wnioskowania przez podatnika do organu rentowego o niepomniejszanie o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek. Są też w tym projekcie zawarte zmiany, które doprecyzowują i uzupełniają obowiązujące przepisy. Pani Marszałek! Na koniec chciałbym podkreślić, że zmiany, które są zawarte w tych projektach ustaw, nie mają wpływu na dochody sektora finansów publicznych bądź wpływ ich jest nieznaczny. Wobec powyższego Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość popiera rozwiązania przedstawione przez rząd i będzie głosował za przyjęciem projektów ustaw z druków nr 207 i 351. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie pośle. Oświadczenie w imieniu Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska przedstawi Wysokiej Izbie pani poseł Zofia Czernow. Bardzo proszę. Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska w sprawie projektu ustawy zawartego w drukach nr 207 i 351. Projekt ustawy wprowadza zmiany w siedmiu ustawach, głównie podatkowych. Jakie to są zmiany i czego dotyczą? Ten projekt w większości regulacji poprawia wcześniej uchwalone ustawy, niektóre podjęte w ostatnich 6 miesiącach. To wszystko spowodowane jest nadmiernym pośpiechem podczas procesu legislacyjnego, który w ostatnich latach nie spełnia podstawowych wymogów i zasad, jakie są niezbędne przy tworzeniu dobrego, stabilnego prawa. Powoduje to wiele poważnych problemów w stosowaniu tego prawa i powstaje wiele błędów i nieprawidłowości. Są one na porządku dziennym i podatnicy mają z tym ogromne kłopoty. Jak zatem w takiej sytuacji budować zaufanie Polaków do państwa prawa? Przechodzę do konkretów. Pierwszym celem procedowanej ustawy jest dostosowanie przepisów o podatku dochodowym do nowej Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, która weszła w życie 1 stycznia 2016 r. Sama propozycja dostosowania przepisów nie budzi wątpliwości. Jest to konieczne, gdyż stan obecny jest bardzo uciążliwy dla podatników, którzy zmuszeni są do samodzielnej interpretacji odmiennych regulacji prawnych. Powstaje jednak pytanie, dlaczego trwało to tak długo. Rząd potrzebował aż 4 lat, aby uzgodnić z Głównym Urzędem Statystycznym dostosowanie przepisów o Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług do prawa podatkowego. Jest to absolutnie niezrozumiałe, bo wszyscy tu siedzący, na tej sali, wiemy, że w Sejmie było dużo czasu, aby tym się zająć, ale rząd odkładał ten problem, odkładał tę sprawę. Kolejna bardzo ważna sprawa dla podatników. Projekt ustawy zawierał - podkreślam: zawierał - także kwestię szerokiego wykorzystywania usługi pocztowej do doręczeń wydruków elektronicznych dotyczących spraw skarbowych. Operator pocztowy oraz osoby działające w jego imieniu uzyskują szeroki dostęp do informacji objętych tajemnicą skarbową. Jednocześnie nie przewiduje się żadnych zabezpieczeń i środków ochrony tych danych, które należą do szczególnie wrażliwych. O wielkim ryzyku wycieku danych stanowiących tajemnicę skarbową świadczą chociażby ostatnie wydarzenia dotyczące kart do głosowania.

Trzeba jednak naprawić ten błąd. Nie możemy narażać Polaków na takie ryzyko. Dlatego wnoszę w imieniu Koalicji Obywatelskiej poprawkę dotyczącą wykreślenia tego punktu z ustawy o COVID-19. Znaczna część projektu ustawy poświęcona jest naprawianiu błędów, usuwaniu oczywistych omyłek, wprowadzaniu uściśleń. Kilka przykładów. Mamy dostosowanie art. 294 Ordynacji podatkowej do przepisów ustawy o działach administracji rządowej. Ostatnio często zmienialiśmy tę ustawę. Natomiast pojawiły się błędy. W ustawie o VAT nastąpiła zmiana błędnej nazwy szefa Krajowej Informacji Skarbowej na właściwą. Jest zmiana w Ordynacji podatkowej poprzez rozszerzenie definicji deklaracji, która obecnie budzi wiele wątpliwości dotyczących statusu prawnego sprawozdań itd. Tych przykładów jest wiele, nie będę ich omawiać. Ale po prostu świadczy to o wielkim pośpiechu, o wielkim bałaganie i błędach. Te błędy i niejasności nie zdarzyłyby się, gdyby dołożono większej staranności podczas prac legislacyjnych. Ze zdumieniem czytam w uzasadnieniu, cytuję: Oceniając wpływ projektowanej ustawy w zakresie ustawy o VAT na mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców, należy wskazać, że proponowana zmiana będzie wymagała od podatników większej staranności w zakresie doboru kontrahentów oraz weryfikacji ich statusu podatkowego, co wpłynie na zwiększenie zaangażowania czasu podatnika w zakresie wypełniania obowiązków podatkowych. Uzasadnia się również, w uzasadnieniu czytamy, że to przyczyni się do uproszczenia i uszczelnienia systemu podatkowego, co absolutnie nie ma z tym nic wspólnego i w tym projekcie to w ogóle nie występuje. Prawo podatkowe powinno być stabilne, jasne i zrozumiałe, nie budzić wątpliwości interpretacyjnych. O takie prawo upominają się podatnicy. Szanujmy prawa podatników. Dziękuję, pani poseł. W imieniu klubu parlamentarnego Lewica głos zabierze pani poseł Monika Falej. Bardzo proszę. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić w imieniu klubu Lewicy stanowisko w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku. Zaproponowane w projekcie rozwiązania można podzielić na trzy grupy przepisów. Po pierwsze, są to przepisy mające na celu dostosowanie przepisów o podatku dochodowym do nowej Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług z 2015 r. Druga grupa to przepisy ograniczające liczbę rocznych obliczeń podatkowych, tzw. PIT 40-A, sporządzonych przez organy rentowe dla podatników, u których z obliczenia organu rentowego wynika nadpłata podatku, oraz przepisy kompleksowo regulujące kwestie wnioskowania przez podatnika do organu rentowego o niepomniejszanie o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek. Zmiana rozszerza skuteczność złożonego przez podatnika wniosku na lata następne, aż do jego wycofania, a także wskazuje, że organ rentowy ma obowiązek uwzględnienia złożonego wycofania wniosku w miesiącu jego złożenia przez podatnika lub najpóźniej w miesiącu następnym. Trzecia grupa to pozostałe zmiany uzupełniające i doprecyzowujące obowiązujące przepisy. Zatrważa fakt, iż rządowy projekt o regulacjach podatkowych trafia pod głosowanie dopiero dzisiaj, niemal w ostatniej chwili.

Na skutek zaniechań przedmiotowej zmiany od 1 stycznia 2021 r. nie byłoby podstawy do odwoływania się w przepisach podatkowych do nowej klasyfikacji. Jest to ustawa czysto techniczna, dostosowująca przepisy podatkowe usprawniające działania rozliczeniowe, choć nie poprawia samej przejrzystości przepisów podatkowych, a wręcz je zaciemnia. Reguluje szczegółowe zapisy. Rząd przedstawia tę ustawę po ponad 4 latach oczekiwania na regulacje. Lepiej późno niż wcale. Z przykrością jednak należy odnotować, że jest to kolejny akt prawny, co do którego pojawiają się wieloobszarowe zapytania, wobec którego występują niejasności. Jest to słaby legislacyjny projekt. Na etapie konsultacji środowiskowych wiele branż zgłaszało postulaty dotyczące zmian i doprecyzowania zapisów.

Prawo musi służyć obywatelom i obywatelkom. Przedsiębiorcy oczekują prostego systemu podatkowego. Jakość prawa to także jego jasność i precyzja oraz czas jego wprowadzenia. Dziękuję bardzo.

Szanowni Państwo! Omawiany dziś projekt ustawy dotyczy ważnego obszaru naszego życia obywatelskiego, społeczno-ekonomicznego. Otóż dokonuje pewnego porządkowania spraw podatkowych w szeregu ustaw z tej dziedziny: ustawa PIT-owska, ustawa dotycząca CIT, Ordynacja podatkowa, ustawa o ryczałcie czy VAT-owska. Generalnie jest to ustawa techniczna, choć przy okazji warto o pewnych rzeczach powiedzieć, bo to nie jest tylko dostosowanie przepisów podatkowych do nowej Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, która została przyjęta w 2015 r., a więc czas przygotowania, o czym już posłowie wspominali, był wyjątkowo długi. Szkoda, że teraz to czynimy w pewnym pośpiechu, ale takie jest życie. Tak jak mówiłem, ta ustawa nie ma charakteru merytorycznego, nie wpływa na zmiany zasad opodatkowania.

Stąd ważne, że ta ustawa da szansę na zmniejszenie liczby rocznych obliczeń podatku PIT czy wprowadza szereg uzupełnień i doprecyzowuje przepisy.

Wreszcie pewne przepisy są wprowadzane na okres obowiązywania stanu epidemii, co jest słuszne.

Oczywiście resort finansów wyjaśnia, że te zmiany były konsultowane i były znane przedsiębiorcom i wychodzą naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, a więc trzeba mieć nadzieję, że ten proces wdrażania będzie dużo, dużo lepszy niż sam proces przygotowania, który został bardzo mocno przeciągnięty, co zapewne nie służy procedurze, ale miejmy nadzieję, że przyczyniło się to do zwiększenia poprawności. Popieramy poprawkę zgłoszoną przez panią poseł. W imieniu Koła Poselskiego Konfederacja głos zabierze pan poseł Janusz Korwin-Mikke. Bardzo proszę, panie pośle. Pani Marszałek! Wysoka Izbo!

Zajączka, który w jego imieniu wygłosił mowę tronową, w której było jedno zdanie o podatkach. Brzmiało ono następująco: materia podatkowa jest rzeczą trudną i ważną, ale najważniejsza jest stabilność, dlatego będziemy uważnie obserwowali rozwój sytuacji i po roku wydamy ustawę, która już nigdy nie będzie zmieniona.

Mój przedmówca powiedział, że to jest taka ustawa porządkująca, mimo to jednak zawiera istotne zmiany.

Konfederacja nie wie, czy ustawa podatkowa po tej zmianie będzie lepsza czy gorsza od poprzedniej, w związku z czym wstrzymamy się od głosu, bo nie możemy tego ocenić.

Nadmierne podatki niszczą ją całkowicie, a podatki dochodowe są najgorszym rodzajem podatków, bo one karzą za pracę. Jak ktoś pracuje, to płaci podatek. My jesteśmy przeciwko tego typu filozofii. Kolega Urbaniak to dokładnie jeszcze, mam nadzieję, wyjaśni. Dziękuję bardzo, panie pośle. Bardzo proszę.

Szanowni Państwo! Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o podatku dochodowym od osób prawnych... od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - już sama nazwa jest skomplikowana. Cóż, zasadnicze zmiany, jakie tutaj zachodzą, to umożliwienie np. niestosowania przepisów dotyczących odpowiedzialności w przypadku dokonania przez podatników płatności na rachunki, które nie są tymi oficjalnymi rachunkami zgłoszonymi do urzędów państwowych, np. w wypadku VAT-u. W porządku, to jest na plus. To w porównaniu z tym, co jest w dzisiejszym stanie prawnym, jest na plus. Wprowadzenie możliwości przekazywania np. paragonów drogą elektroniczną również jest usprawnieniem, w porządku. Problem jednak leży zupełnie gdzie indziej. Po pierwsze, o czym już wspomniał mój przedmówca - pan Janusz Korwin-Mikke, zmieniacie podatki, zmieniacie prawo setki razy. A sami przedsiębiorcy - i wasz rząd doskonale o tym wie. Ja sam reprezentuję Pomorze, rozmawiam z przedsiębiorcami, na tych samych rozmowach był nawet np. minister Sellin. Rozmawiamy i podstawowym problemem, jaki też teraz, w dobie kryzysu, jest i który widzą przedsiębiorcy, jest split payment, który wprowadziliście, czyli właśnie podzielona płatność, utrzymanie części pieniędzy w bankach, dzięki czemu banki mogą nimi obracać i pożyczać pieniądze rządowi. A druga sprawa to metoda kasowa naliczania podatków. Pomyślcie troszeczkę i skorzystajcie z tego, o czym sami przedsiębiorcy wam mówią. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do pytań. Wyznaczam czas - 1 minuta. Bardzo proszę. Wysoka Izbo! Procedowany projekt może wyglądać na nudny i niewinny, ale PiS nie byłby sobą, gdyby nie wsadził tu jakiejś miny. W tej ustawie proponowano przekazanie tajnych danych skarbowych obywatelek i obywateli Poczcie Polskiej. Zrobiona tak nie dlatego, że był zły, ale dlatego, że wcześniej już tę wrzutkę udało się przepchnąć w pierwszej ustawie o COVID. Dziś Poczta Polska ma już nasze PESEL-e, tajne dane skarbowe, może i numery butów. Dziś rano podczas kontroli, którą przeprowadziłam w UODO z posłanką Moniką Falej, stwierdziłyśmy ze zdziwieniem, że instytucja ta, przeznaczona do ochrony danych osobowych, nic nie wie o tym, co się dzieje z naszymi danymi po przekazaniu ich Poczcie Polskiej.

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!

Rozliczenia podatkowe to często mniej lub bardziej przykry obowiązek w przypadku wielu działalności gospodarczych. W czasie kryzysu kluczowa jest natomiast płynność finansowa. Dlatego Lewica złożyła projekt ustawy o dofinansowaniu kosztów stałych przedsiębiorców w warunkach zagrożenia ekonomicznego w następstwie wystąpienia koronawirusa. Projekt zakłada dofinansowanie kosztów stałych przedsiębiorców z budżetu państwa do kwoty nieprzekraczającej 50 tys. zł miesięcznie przez okres 6 miesięcy. Chciałbym zapytać: Jakie jest stanowisko ministerstwa w sprawie tej ustawy i jakie zajmie stanowisko podczas prac sejmowych? Proszę o odpowiedź na piśmie. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Witam koleżanki i kolegów posłów. Nikt nie lubi płacić podatków, ani osoby fizyczne, ani podmioty gospodarcze, ale jeżeli już się płaci, to chce się mieć poczucie, że rząd właściwie korzysta z pieniędzy, jak również poczucie - i to jest niesłychanie ważne - trwałości rozwiązań prawnych. Zmieniamy dzisiaj siedem ustaw. Jak już się coś skończyło, to rząd próbuje nadganiać. Mówimy tutaj, nie będę powtarzał, o międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług. Ona wygasła z końcem poprzedniego roku. Tak samo jest z PIT-em.

To jest fatalne dla gospodarki, fatalne dla osób fizycznych. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Zmiana goni zmianę. Poprawiamy dzisiaj przepisy, które dopiero co przyjmowaliśmy. W gruncie rzeczy - konia z rzędem temu, kto nadąża za tymi zmianami. Ale w tym kontekście coraz większego znaczenia nabiera zalegająca nie wiadomo gdzie i nie wiadomo dlaczego nowa Ordynacja podatkowa.

Warto ją odkurzyć i o to apeluję, zwłaszcza że dzisiaj przydałyby się rozwiązania, które były zawarte przynajmniej w pierwszej wersji tej ordynacji, dotyczące informacji. Chodzi o niewładcze formy funkcjonowania administracji podatkowej, takie jak informacja, konsultacje, porozumienie urzędnika skarbowego z przedsiębiorcą (Dzwonek) i ochrona prawna podatnika, który do tej informacji, tej konsultacji czy tego porozumienia. by się zastosował. Pytam: Kiedy ta ordynacja trafi wreszcie do Sejmu?

Pani Marszałek! Panie Ministrze! Ja mam proste i zwykłe pytanie: Czy Poczta Polska stała się jakąś specjalną służbą, która ma inwigilować obywateli na rzecz rządu? Najpierw przekazaliście Poczcie Polskiej wszystkie nasze dane osobowe, łącznie z numerami PESEL, co z niewiadomych względów pominął milczeniem prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Teraz okazało się, przy okazji tej ustawy, że dostali również dostęp do tajemnicy skarbowej, czyli do wszystkich dokumentów, które wysyłamy do skarbówki, do wszystkich danych dotyczących naszych kontroli. W jakim celu Poczta Polska ma mieć dostęp do takich informacji, zresztą nie tylko Poczta Polska, ale także wszystkie agencje, które działają na jej rzecz? Dziękuję. Bardzo proszę.

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Zwłoka przy tej ustawie to jest słowo klucz. Ta zwłoka to jest kilka lat zwlekania z tymi uregulowaniami. Ale ona w kontekście podatkowym nabiera zupełnie innego i szerszego znaczenia. Panie Ministrze! Od wielu miesięcy, od wielu tygodni przedsiębiorcy skarżą się na to, że środki, które przeznaczają na VAT, zarówno w podzielonej płatności, jak i w innej formule, tradycyjnej, zalegają na kontach urzędów skarbowych i urzędy skarbowe robią wszystko, żeby zarówno w tym trybie przyspieszonym, jak i w trybie zwykłym nie dokonywać zwrotu środków, które właśnie pochodzą z podatku VAT. I pytanie jest takie: Czy prawdą jest, że to jest na skutek instrukcji z Ministerstwa Finansów, które zmierzają do tego, żeby jak najmniej zwracać przedsiębiorcom VAT-u? Tak jak mówię, dzieje się to zarówno w tym przyspieszonym trybie, jak i w trybie zwykłym.

Bardzo proszę. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Zacytuję trzy fragmenty z państwa uzasadnienia ustawy: Projekt ustawy ma na celu usunięcie nieścisłości w ustawie o VAT z sierpnia 2019 r., doprecyzowanie przepisów Ordynacji podatkowej dotyczących indywidualnych rachunków podatkowych i - mój taki ulubiony, bo chyba najbardziej zawiły - usunięcie nieścisłości powstałej na skutek uchwalenia ustawy nowelizującej z 9 sierpnia 2019 r. Nie mam pretensji do państwa, że państwo chcą to usystematyzować, ale mam pytanie o odpowiedzialność polityczną. Nie ma nic gorszego niż zatrudnianie ekspertów do tego, żeby wciąż analizowali nowe prawa. Jeśli co chwilę pojawiają się nowe prawa, a tu mamy nowelizację ustaw z 2019 r., czyli dopiero co. Zmiany w siedmiu ustawach. Jeżeli to tak będzie w kółko funkcjonowało, [[Dzwonek]] to każdy przedsiębiorca będzie obciążony tym, że musi kolejne osoby zatrudniać do analizowania i interpretowania ustaw. Bardzo proszę. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Obecnie zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej istnieją dwa rodzaje doręczeń pism: pierwszy - za pokwitowaniem, drugi - za urzędowym poświadczeniem odbioru. Celem opisywanych zmian, widocznym w obu ustawach, jest wprowadzenie usługi hybrydowej, co skutkuje umożliwieniem operatorowi pocztowemu oraz jego pracownikom wglądu do przesyłek zawierających informacje objęte tajemnicą skarbową. W związku z tym mam pytanie: Dlaczego po raz kolejny w ostatnim czasie wprowadza się regulacje umożliwiające operatorowi pocztowemu wgląd do informacji wrażliwych? Czy chcemy, aby pracownicy operatora pocztowego posiadali informacje objęte tajemnicą skarbową? No i najważniejsze pytanie: Czy jest to kolejny element inwigilacji Polek i Polaków? Panie pośle. Kolejne pytanie zada pani poseł Marta Wcisło, Koalicja Obywatelska. Bardzo proszę. Wysoka Izbo! Kolejny projekt ustawy, zmian w podatku w Polsce.

Część z tych zmian wynika z epidemii, jest uzasadniona, część to poprawki. Ale niektóre zapisy uzasadnienia ustawy o podatku VAT budzą moje zaniepokojenie, ponieważ czytamy, że wymaga się od podatnika większej staranności w zakresie doboru kontrahentów oraz weryfikacji ich statusu podatkowego. Pytam: Czy to jest rola przedsiębiorcy - weryfikować? Czy przedsiębiorca ma pracować, zarabiać, czy weryfikować? A może ma wyposażyć się w wykrywacz kłamstw? Jak ma to robić? To nie jest rola przedsiębiorcy. Z mojego doświadczenia, ponaddwudziestoletniego, w zakresie prowadzenia działalności nie wiem, jak weryfikować kontrahentów, [[Dzwonek]] którzy mogą mieć status dobrego podatnika bądź nie. Dziękuję, pani poseł. I pan poseł Michał Szczerba, Koalicja Obywatelska. Ale bardzo proszę o wyciszenie rozmów w ławach, bo naprawdę bardzo mocno się roznosi państwa głos, a przeszkadzacie swoim kolegom i koleżankom klubowym, chciałam zauważyć. Bardzo proszę, panie pośle. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Trzeba bić na alarm. Operator pocztowy Poczta Polska uzyskuje dostęp do informacji objętych tajemnicą skarbową. Poczta Polska ma w tej chwili nasze PESEL-e, ma pełne informacje dotyczące wielu wrażliwych kwestii dotyczących każdego i każdej z nas, ma w wielu przypadkach już dostęp do spisu wyborców, mimo że Kodeks wyborczy mówi wprost: spis wyborców sporządza się wyłącznie w dwóch egzemplarzach - dla gminy i dla komisji obwodowej. W tej chwili chcecie wyposażyć tę spółkę Skarbu Państwa w dane, informacje objęte tajemnicą skarbową. Jest to bardzo niebezpieczne. Również bardzo niebezpieczne jest to, że każdego dnia wydatkowane są miliony złotych na przygotowanie Poczty Polskiej do wyborów 10 maja.

Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Wysoka Izbo! Przyzwyczailiście już podatników VAT do regularnych zmian przepisów. Zanim nauczą się prawidłowo zastosować jeden przepis, pojawia się nowy lub aktualizacja tego, co niedawno wprowadzono. Niestety tak stanowi się prawo w tej Izbie, jednak wprowadzając tą ustawą klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania w odniesieniu do zaliczania kosztów hipotetycznych odsetek do kosztów uzyskania przychodów, dokręcacie śrubę przedsiębiorcom, szczególnie teraz, kiedy mamy czas pandemii, która w dużym stopniu dotknęła właśnie osoby prowadzące działalność gospodarczą. Kolejna sprawa to doręczanie pism za pomocą usługi hybrydowej. W jaki sposób zagwarantujecie bezpieczeństwo przekształcania dokumentu elektronicznego w przesyłkę listową przez operatorów? Czy dane przetwarzane będą zgodnie z wytycznymi [[Dzwonek]] zapewniającymi stosowanie RODO? Bardzo proszę. Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! Złożyliśmy poprawkę do tego projektu ustawy, która wykreśla tę usługę pocztową. Rezygnujemy z usługi pocztowej w zakresie dostarczania wrażliwych danych skarbowych podatnikom. Zdaje sobie pan sprawę z tego, że ta dostępność danych, ta poufność nie jest w żaden sposób zabezpieczona. Nie ma żadnych środków ochrony. Uważam, że należy przychylić się do naszej poprawki - o co bardzo apeluję - i w międzyczasie dostosować prawo w taki sposób, aby nasze dane skarbowe były bezpieczne. Co się stanie, jeżeli dojdzie do takiego skandalu, wycieku danych skarbowych wynikającego z usługi Poczty Polskiej? Jakie będą konsekwencje? Jaka będzie wiarygodność [[Dzwonek]] polskiego rządu i polskiego Ministerstwa Finansów?

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Omawiany projekt ustawy m.in. doprecyzowuje istniejące przepisy czy usuwa pozostałe wątpliwości. Przedsiębiorcy cały czas narzekają na to, że tworzone jest prawo, które jest niejasne. Dobrze, że czasami przychodzi refleksja i pewne regulacje są korygowane. W związku z powyższym mam do rządu następujące pytanie: Czy nie można od razu tak przygotować przepisów, aby nikt nie miał wątpliwości, o co chodzi? Dziękuję, pani poseł. Bardzo proszę.

Wysoka Izbo!

W tej ustawie, proszę państwa, m.in. zajęto się wyrobami rękodzieła ludowego typu bielizna, z wyłączeniem jednakowoż biustonoszy, gorsetów, szelek, pasów do pończoch itd. - w ustawie (Dzwonek), brawo - a z drugiej strony jest transport, uwaga, lotniczy i kosmiczny. Czytając, że transport lotniczy i kosmiczny. Perspektywicznie myślący ustawodawca przewiduje, że będzie w Polsce ten transport kosmiczny, na co ja się bardzo cieszę.

Przypomniało mi się, że.

Pan poseł Tadeusz Tomaszewski, klub Lewica. Bardzo proszę. Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Szanowny Panie Ministrze! Przy okazji debaty o ustawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych chciałbym zapytać o stan prac w Ministerstwie Finansów dotyczących stworzenia możliwości prawnej podziału 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na więcej niż jedną organizację pozarządową. Za rok 2018 w 2019 r. podatnicy przekazali 875 mln zł, 14,5 mln podatników skorzystało z tej możliwości.

Wielu podatników teraz w okresie sprawozdawczym pyta, czy mogą przekazać swój 1% na więcej niż jedną organizację.

Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie pośle. W imieniu rządu na pytania odpowie podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów pan minister Jan Sarnowski. Bardzo proszę.

W pierwszej kolejności chciałem odnieść się do problemu, który był zgłaszany najczęściej, w związku z którym zgłoszona została poprawka, mianowicie do kwestii Poczty Polskiej, która jakoby miałaby mieć dostęp do tajnych danych skarbowych. Niektórzy z państwa posłów również zadawali pytania, w jaki sposób paczki czy listy dostarczane przez Pocztę Polską będą zabezpieczane przed ich otwarciem oraz zapoznaniem się z ich zawartością przez pracowników poczty.

Tak że drogą wstępu, proces, który zostanie wszczęty we współpracy z Pocztą Polską, będzie całkowicie bezpieczny i nie doprowadzi do tego, że osoby niepowołane będą miały dostęp do informacji podatkowych podatników. W systemie Krajowej Administracji Skarbowej tworzone jest pismo do podatnika. Tam pismo to jest podpisywane, a następnie za pośrednictwem szyfrowanego łącza jest przesyłane na dedykowany szyfrowany serwer Poczty Polskiej wraz z tzw. plikiem sterującym. Plik sterujący zawiera informację, pod jaki adres należy doręczyć przesyłkę i z ilu stron ona się składa. Z tego serwera automat Poczty Polskiej pobiera plik i wysyła go do maszyny drukująco-kopertującej. Maszyna ta drukuje pismo, składa je i umieszcza w kopercie, którą zamyka. Z pliku sterującego maszyna drukuje również adres umieszczony na kopercie. W ciągu minuty drukowanych i kopertowanych będzie nawet kilkaset tego rodzaju przesyłek. Po wykonaniu usługi plik zawierający dane objęte tajemnicą skarbową jest usuwany z serwera. W ciągu całego procesu nie ma fizycznej możliwości zapoznania się przez pracownika Poczty Polskiej z zawartością listu. Do takiej sytuacji mogłoby potencjalnie dojść jedynie w przypadku awarii maszyny drukująco-kopertującej, np. w przypadku zacięcia się papieru.

Proces jest automatyczny i całkowicie bezpieczny. Uprzejmie prosimy o odrzucenie zgłoszonej przez państwa poprawki. Czy zadaniem przedsiębiorcy jest monitorowanie osób, z którymi współpracuje, i upewnianie się co do ich rzetelności podatkowej? Zdaniem Ministerstwa Finansów kluczowe, szczególnie teraz, w czasach COVID-19, jest skupienie się przedsiębiorcy na prowadzeniu działalności gospodarczej.

Tu również trzeba zaoponować.

Co do zasady średni czas oczekiwania na uwolnienie środków to 10 dni. Tak że w sytuacji, gdy nie ma żadnych wątpliwości, można powiedzieć, że środki uwalniane są praktycznie z dnia na dzień. Średnią podnosi pewna liczba podatników, w stosunku do których rzeczywiście wątpliwości się pojawiają.

Tak że nie jest to wcale złoty środek i narzędzie ratunku dla przedsiębiorców (Dzwonek), wręcz przeciwnie, to miecz obosieczny, który może jeszcze bardziej pogorszyć ich sytuację.

Od początku tego roku funkcjonuje ulga na złe długi, którą dodatkowo zmieniono na czas COVID-u tak, żeby w szczególny sposób chroniła wierzycieli.

Co więcej, wierzyciel może tego dokonać nie w normalnym terminie 3 miesięcy, ale miesiąca. Ordynacja podatkowa - projekt nie zginął. Z uwagi na zasadę dyskontynuacji prac Sejmu projekt znów będzie musiał przejść całą ścieżkę rządową. Biorąc pod uwagę palące potrzeby związane z epidemią COVID-19, moment, w którym to będzie zrealizowane, jest aktualnie w pewien sposób odsuwany w czasie, natomiast wciąż jest to jeden z priorytetów Ministerstwa Finansów. Co do PKWiU, dostosowania zmiany tej z roku 2008 na tę z 2015 - rzeczywiście jest to zmiana techniczna, natomiast jest to zmiana techniczna, która była odsuwana w czasie, biorąc pod uwagę bardzo wiele innych projektów realizowanych w tym czasie w Ministerstwie Finansów.

W sumie według różnych obliczeń, również dokonywanych w Ministerstwie Finansów, różne ulgi i obniżki podatków doprowadziły do zmniejszenia wpływów budżetowych Polski o ok. 20 mld zł. To jest 20 mld zł, które pozostały w kieszeniach podatników dzięki obniżkom podatków. Odnośnie do podziału 1% dla organizacji pożytku publicznego na więcej niż jedną organizację prace w tym zakresie toczą się już w Ministerstwie Finansów, prowadzimy badania dotyczące europejskiego i światowego benchmarku, innych krajów, dotyczące tego, na jaką liczbę organizacji jest otwarta możliwość podziału tego 1%. Wprowadzone zostały w różnych krajach też pewne holdy dotyczące minimum przekazywanego 1%, który mógłby podlegać podzieleniu. Mamy również nadzieję, że te prace zakończą się jak najszybciej i wprowadzimy tę możliwość już od przyszłego roku podatkowego, czyli dla rocznego rozliczenia za rok 2020. Dziękuję bardzo, panie ministrze. Zamykam dyskusję. W związku z tym, że w czasie drugiego czytania zgłoszono do przedłożonego projektu ustawy poprawki, proponuję, aby Sejm ponownie skierował ten projekt do Komisji Finansów Publicznych w celu przedstawienia sprawozdania. Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę.